Wielokrotnie słyszeliśmy na tej sali słowa otuchy, słowa, które miały zachęcić opozycję do konstruktywnej współpracy. Nie ukrywam, że nawet niektórzy z nas w to uwierzyli, ale rzeczywistość jest zupełnie inna. Otóż nie tylko wniosek Lewicy, i inne, spada z porządku posiedzenia Komisji Finansów Publicznych, ale też posiedzenie bez żadnych formalnych czy nieformalnych, merytorycznych wniosków zostaje przerwane.

Panie pośle, jest ogłoszona przerwa w posiedzeniu komisji. Osobiście rozmawiałam z panem marszałkiem Czarzastym, informując go o tym, o godz. 10. Ale wniosek jest już nieaktualny, ponieważ komisja już działa od godz. 12. W tej chwili jest ogłoszona przerwa.

Wniosek formalny, proszę bardzo. Szanowna Pani Marszałek! Chciałbym złożyć wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o nowy punkt.

Chodzi o osoby, które tak naprawdę są zamknięte, są to osoby zakażone, wraz z personelem. To są już setki osób. My musimy mieć dzisiaj, pani marszałek, informację premiera i minister rodziny o tym, co w takich sytuacjach robić. Nie można tych ludzi zostawić samym sobie na czas Wielkiejnocy.

To jest trzeci dzień posiedzenia Sejmu. Wczoraj takiego wniosku nie było.

Bardzo proszę.

Proszę państwa, został zgłoszony wniosek o przerwę - tylko o przerwę, ponieważ druga część tego wniosku była nieregulaminowa. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za zarządzeniem przerwy w obradach, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Sejm wniosek odrzucił. Komisja Finansów Publicznych przedłożyła sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz o poselskim projekcie ustawy o utworzeniu prawdziwej Tarczy antykryzysowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, druk nr 332. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego sprawozdania. Proponuję, aby w tym przypadku Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 51 pkt 3 regulaminu Sejmu oraz w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłuchał 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycje przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Proszę bardzo. Zwracam się do pani marszałek o to, aby ogłosiła przerwę i zwołała Konwent Seniorów, aby dać szansę przybycia na nasze obrady ministrowi finansów. Za chwilę będziemy słuchali sprawozdania komisji finansów, które w istocie będzie skutkowało różnymi wydatkami budżetowymi. Ktokolwiek słyszał, ktokolwiek wie, gdzie jest minister finansów, niech zaprosi pana ministra na obrady Wysokiej Izby. Z ust prezesa Narodowego Banku Polskiego słyszeliśmy, że mamy nieprzebrane ilości gotówki. Kiedy posłowie opozycji składają wniosek, aby wprowadzić stan klęski żywiołowej, słyszymy, że doprowadzilibyśmy do ruiny budżetu państwa. A więc od eldorado do ruiny jeden krok.

Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Finansów Publicznych mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie z rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, druk nr 330, oraz poselskiego projektu ustawy o utworzeniu prawdziwej Tarczy antykryzysowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, druk nr 324. Sejm po przeprowadzeniu dyskusji podczas pierwszego czytania skierował obydwa projekty do Komisji Finansów Publicznych.

Część poprawek została przyjęta, m.in. poprawki, które uwalniały ten projekt od zapisów dotyczących zmian w ustawach systemowych.

Zostały również przyjęte rozwiązania z projektu poselskiego: trzy artykuły, praktycznie w całości, z modyfikacją, za zgodą oczywiście wnioskodawców i autorów tego projektu. Ostatecznie komisja rekomenduje przyjęcie projektu zawartego w sprawozdaniu w druku nr 332. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Premierze! Jesteśmy świadkami kryzysu pandemii, jesteśmy świadkami kryzysu gospodarczego, który się pogłębia, ale jesteśmy również świadkami kryzysu państwa. Ten kryzys państwa widać w bardzo wielu obszarach. Sytuacja w szpitalach, generalnie w całej służbie zdrowia, jest bardzo dramatyczna. Otrzymujemy setki, tysiące sygnałów o tym, jak trudna jest w tej chwili sytuacja pracowników medycznych, jakie są kolosalne braki, jeśli chodzi o wyposażenie szpitali, środki ochrony osobistej. To wszystko sprzyja dalszemu rozprzestrzenianiu się epidemii. To są bardzo poważne sprawy. O pomoc proszą samorządy, o pomoc proszą przedsiębiorstwa. Wszystko to pokazuje, że dotychczasowe działania rządu po prostu nie spełniają oczekiwań. Nie spełniają oczekiwań m.in. dlatego, że rząd przyjął sposób pracy, który niestety urąga najlepszym zasadom pracy legislacyjnej i rządzeniu państwem w czasach trudnych, w czasach kryzysu.

Wczoraj mieliśmy kolejny przykład ustawy, która ma pomóc przedsiębiorcom, ale w istocie rzeczy w ogromnej swojej części stanowi zbiór przepisów czysto proceduralnych, dotyczących trybu komunikowania się, postępowań, natomiast jeśli chodzi o pomoc dla przedsiębiorców, pomoc dla pracowników, pomoc dla gospodarki, to można na palcach jednej ręki policzyć zapisy, które przynoszą ulgę finansową, ekonomiczną gospodarce znajdującej się w kryzysie. Już wspominałem wczoraj podczas dyskusji, że skandalem jest, że procedujemy nad ustawą, która zmienia 60 innych ustaw. Jest to po prostu taki omnibus, w którym znalazły się zmiany najdziwniejszych przepisów, niemających często w ogóle nic wspólnego z tym, czym się powinniśmy zajmować, to znaczy walką z pandemią i ratowaniem gospodarki. Do szczególnych takich klejnotów, które nam się udało znaleźć podczas tych nocnych obrad, należy zapis dotyczący Polskiego Związku Łowieckiego, gdzie przesuwa się terminy wyborów władz Polskiego Związku Łowieckiego ze względu na epidemię. Poparliśmy ten zapis, mimo że oczywiście on nie ma większego związku z tym, czym się powinniśmy zajmować. Pojawiły się dziwne inne wrzutki zwalniające operatorów telefonii komórkowych z wypełniania pewnych zobowiązań, uchylające obowiązek posiadania opinii środowiskowej itd., itd. Mieliśmy wrażenie, że przy okazji tej ustawy realizowane są różne dziwne partykularne interesy. Nie mogliśmy się temu oczywiście przyjrzeć z dostateczną starannością, bo nie było czasu. Pracowaliśmy, jak powiedział pan przewodniczący, do godz. 4 rano, ale mimo to istnieje duże ryzyko, że w tej ustawie znalazła się cała masa zapisów, które są po prostu szkodliwe. Ale co najważniejsze - pomoc, którą miała nieść ta ustawa, jest po prostu niewystarczająca. Odrzuciliście, drodzy państwo, wszystkie nasze poprawki, w tym te najważniejsze. Jeszcze raz je przypomnę. Chcemy 20 mld zł na służbę zdrowia. To jest 1% PKB. Jeżeli w ogóle mamy poważnie myśleć o tym, żeby dogonić kraje europejskie, jeśli chodzi o udział wydatków na zdrowie w Unii Europejskiej, to musimy to zrobić. I akurat jest czas taki, kiedy to służba zdrowia potrzebuje pieniędzy najbardziej. To jest sprawa rozciągnięcia wakacji składkowych ZUS na wszystkie przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie. Nie powinniśmy w tej kategorii przedsiębiorstw dyskryminować. Wszystkie te firmy potrzebują pomocy. Po trzecie, to jest zapewnienie zasiłków opiekuńczych również dla tych rodziców, którzy mają dzieci w wieku do 15 lat. Tego naprawdę nie jestem w stanie zrozumieć, panie premierze, niech pan mi wyjaśni, dlaczego pan odmawia zgody na ten zapis. Mówicie, że nie ma pieniędzy na te propozycje, więc ja wam chcę wskazać kilka bardzo jasnych dróg, jak można te pieniądze zdobyć. Zrezygnujcie z paru megalomańskich projektów inwestycyjnych i skupcie się na tym, co jest naprawdę ważne dla Polski. A oprócz tego są pieniądze europejskie i przestańcie uprawiać antyeuropejską propagandę, dlatego że to jest działanie, które powoduje (Dzwonek), że na Kremlu biją brawo.

Szanowna Pani Marszałek! Panowie Ministrowie! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15 chciałbym przedstawić stanowisko w sprawie druku sejmowego nr 332 zawierającego sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o dwóch projektach dotyczących ochrony de facto dzisiaj zdrowia Polaków, ale również sytuacji naszej gospodarki, sytuacji ekonomicznej wielu Polaków. Faktycznie, tak jak pan przewodniczący zauważył, posiedzenie Komisji Finansów Publicznych było burzliwe, było długie, natomiast wiele posłanek i posłów odczuwa wielki niedosyt z powodu tej pracy. Uczyniono wiodącym projekt rządowy - projekt, który, tak jak większość głosów wskazuje, jest mało ambitny, jest projektem niewychodzącym naprzeciw oczekiwaniom dzisiaj wielu pracodawców, wielu pracowników. Ubolewam też jako przedstawiciel klubu Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15, że w tak niewielkim stopniu w toku prac skorzystano z niezwykle wielu dobrych pomysłów, które zawiera nasz projekt. Ciągle liczę, powiem szczerze - i mój głos na koniec prac wczorajszych był też dowodem takiej dobrej woli - na to, że w większym stopniu państwo sięgniecie po te naprawdę dobre pomysły, które były wczoraj w całości prezentowane przez pana prezesa Władysława Kosiniaka-Kamysza, przez pana marszałka Stanisława Tyszkę. To są naprawdę dobre, ambitne pomysły, które będą z pewnością dobrze służyć naszej gospodarce, będą chronić miejsca pracy, a na tym tak naprawdę powinno wszystkim zależeć. Wskażę chociażby na najważniejsze z tych postulatów, które zawierał i zawiera projekt prawdziwej tarczy antykryzysowej. Mówimy w nim o wsparciu dla wszystkich pracowników w wysokości minimalnego wynagrodzenia, z akcentem: dla wszystkich. Nie dzielimy tu na lepszych i gorszych, a niestety trudno odnieść podobne wrażenie w przypadku projektu rządowego. Mówimy również o wsparciu dla wszystkich przedsiębiorców poprzez postulat Koalicji Polskiej dobrowolnego ZUS-u.

Wreszcie, też w przeciwieństwie do projektu rządowego, mówimy o Funduszu Płynności finansowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla wszystkich przedsiębiorców, i tu bez obostrzeń, bo nie można, oferując pomoc, jednocześnie skazywać przedsiębiorców na biurokratyczne bariery. Mówimy także o zwolnieniach z PIT-u i z CIT-u, również bez zbędnych formalności, bez zbędnych problemów. Na te rozwiązania, Wysoka Izbo, Polskę musi być stać. Słyszeliśmy tyle o zrównoważonym budżecie. Wedle bardzo ostrożnych szacunków, bardzo ostrożnych prognoz w Polsce na koniec roku 2020 możemy mieć do czynienia z ok. 2 mln osób pozostających bez pracy.

Naprawdę z dobrą wolą ciągle oferujemy dobre rozwiązania, których w naszym projekcie ustawy jest bardzo wiele. Liczymy na większą otwartość ze strony większości sejmowej.

Koalicja Polska (Dzwonek) tych rozwiązań zaoferowała w swoim projekcie naprawdę bardzo wiele. Bardzo dziękuję, panie pośle.

Wysoka Izbo! Pan marszałek Zgorzelski przywołał tutaj postać nieobecnego ministra finansów. Rzeczywiście w kuluarach zastanawialiśmy się, jak ten dżentelmen, bo w to nie wątpimy, ma na nazwisko. Być może to jest nasza wina, że niedostatecznie dobrze czy nie dość dobrze pamiętamy nazwiska wszystkich wysokich urzędników państwowych, ale rzeczywiście pod tym apelem także i my się podpisujemy: dobrze by było, gdyby minister finansów pojawił się na tej sali, pojawił się przed Polakami, i powiedział, jaki jest stan finansów publicznych. Panie marszałku - zwracam się do marszałka Zgorzelskiego - wydaje mi się, że brakuje tu jeszcze jednej ważnej postaci. Mam na myśli panią Jadwigę Emilewicz, o mało co wicepremiera polskiego rządu, która poprzednią ustawę o COVID-19 pilotowała i gorąco wszystkich zachęcała do tego, żebyśmy ją poparli. Ustawa, nad którą w tej chwili dyskutujemy w trakcie drugiego czytania, jest istotnym uzupełnieniem i rozszerzeniem tamtej inicjatywy pani minister Emilewicz, a jej także, co odnotowuję z zaniepokojeniem, pani marszałek, na tej sali nie ma. Szkoda, żałujemy, ale może to się zmieni. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Podczas wczorajszej debaty sformułowałem cztery kryteria dotyczące dobrej ustawy ratunkowej dla polskiej gospodarki. Pozwólcie państwo, że je przypomnę. Ta ustawa moim zdaniem powinna działać szybko, powinna być prosta, hojna i nie przynosić negatywnych skutków ubocznych. Odnoszę wrażenie, że istotna część tej ustawy to jest jeden wielki skutek uboczny.

Otóż dokonuje się w tej ustawie, nad którą dzisiaj debatujemy, kolejnego zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku sprzedaży i wymiany kryptowalut. Powiedzcie, proszę, jaki to ma związek z walką ze skutkami koronawirusa, ze skutkami gospodarczymi, który to kryzys dewastuje polskie przedsiębiorstwa, który niszczy życie milionów polskich rodzin. Czy to naprawdę jest temat do dywagacji na sali sejmowej, w Komisji Finansów Publicznych? Rozporządzenie ministra finansów, które jest poświęcone opodatkowaniu, a raczej dotyczy braku opodatkowania kryptowalut, traci swoją moc z dniem 30 czerwca. Jeśli chcecie dalej zwalniać handel kryptowalutami z opodatkowania, to zmieńcie to rozporządzenie ministra finansów, a nie angażujcie do tego Wysokiej Izby i nie zaciemniajcie pola widzenia, nie zaciemniajcie obszaru spraw.

To jest dowód jakiejś niebywałej partaniny legislacyjnej. Nie oczekujmy, że przedsiębiorcy, do których ta ustawa jest adresowana, to zrozumieją, jeśli gubią się w tej numeracji i w tej nomenklaturze sami legislatorzy, jak to miało miejsce dziś w nocy w trakcie obrad Komisji Finansów Publicznych. Lewica, pani marszałek, przygotowała pakiet 11 poprawek, które chciałbym złożyć na pani ręce z prośbą o ich uwzględnienie. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję.

Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Ustawa, która została nam zaprezentowana, tzw. tarcza 2.0, to tak naprawdę łata naszywana zaledwie po tygodniu na to, co miało ratować polską gospodarkę, ale niestety jej nie uratuje. To kpina z inteligencji Polaków, to kpina z polskich przedsiębiorców, to także kpina z prawników, jeżeli chodzi o jakość legislacyjną całości tego projektu. Najpierw nie mogliśmy się doczekać projektu. Przypomnę, że w trakcie konsultacji z panem premierem, na które sam pan premier nas zaprosił, obiecano nam, że będziemy mieć co najmniej 1 dzień - 1 dzień, o tyle prosiliśmy - na zapoznanie się z projektami, zanim trafią one do Sejmu. Zostało ono przesunięte o kolejne godziny. Mamy nieustanne przekładanie, właściwie praca Sejmu w ostatnich dniach jest takim chaosem, że ciężko oczekiwać, że z tego Sejmu wyjdzie jakkolwiek dobrze napisane prawo. I chciałbym wierzyć, że w kancelarii premiera i w odpowiednich ministerstwach panuje nieco większy porządek w przygotowywaniu tych przepisów, aczkolwiek ich redakcja na to nie wskazuje. Dziś komisja do wczesnych godzin porannych pracowała nad tym w atmosferze nerwowej, atmosferze pracy zdalnej, podczas której posłowie mieli problem z prawidłowym głosowaniem nad wnioskami i z prawidłowym składaniem poprawek. Konfederacja przygotowała ponad 40 poprawek do tej dziurawej, papierowej, biurokratycznej tarczy antykryzysowej. Zgłaszamy te same poprawki, rozsądne poprawki, które rząd częściowo uznaje, ponieważ znajdujemy prawdziwe luki w tym projekcie, ale później nie chce przegłosować naszych poprawek, tylko zgłasza je jako swoje. No, to już wyjątkowa małość, kiedy znajdujemy jakiś rzeczywisty błąd w projekcie, pomijając jego założenia, z którymi się nie zgadzamy, ale kiedy znajdujemy błędy polityczne, takie, że rząd co innego publicznie deklaruje, a co innego później wpisuje, z powodu najwyraźniej panującego bałaganu, do projektu, to naprawdę wypadałoby już uznać nasze poprawki. A mianowicie w żaden sposób tarcza rządowa nie chroni interesów kredytobiorców i leasingobiorców.

Liczymy na to, że rząd pochyli się nad interesami Polaków, realnymi interesami, a nie będzie zajmował się, tak jak dziś, po raz kolejny drukowaniem na pierwszych stronach gazet wirtualnych kwot typu 200 mld.

To nie jest tarcza 2.0, to nie jest nawet funkcjonalna wersja beta.

Ludzie nie zdążyli jeszcze przebrnąć przez 170-stronicową instrukcję do jedynki, a już wypuszczacie dwójkę. Rozumiem, że w przyszłym tygodniu będzie wersja 3.11, potem XP, Vista itd. W poważnym państwie to wygląda tak, że ktoś budzi premiera w środku nocy i mówi: Panie premierze, jest katastrofa. Jaka katastrofa?

Już po prostu to widzę, jak uchwalamy na szybko specustawę o zaopatrzeniu frontu w przypadku wojny albo nowelizację ustawy o wykonywaniu zawodu żołnierza. Okazuje się, że trzeba mieć jakieś specjalne prawo jazdy na czołgi, a nie przewidzieliśmy, że tego teraz nie da się zrobić, więc wprowadzamy szybko poprawkę, poprawka wchodzi w życie. Tak to będzie wyglądało. I to jest oskarżenie wszystkich państwa, bo państwo miało czas zajmować się, nie wiem, takimi ważnymi przepisami, jak to, jaki VAT nałożyć na pączki w zależności od tego, co w nich jest, jaką powierzchnię lokalu gastronomicznego powinny zajmować okna, jak walczyć z loteriami paragonowymi.

Dziękuję bardzo. Szanowna Pani Marszałek! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w sprawie sprawozdania zawartego w druku nr 332 o projekcie ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Szanowni Państwo!

Oczywiście sytuacja się zmienia, jest dynamiczna i zupełnie inaczej wyglądała 2 tygodnie temu, 3 tygodnie temu, niż wygląda obecnie. Wtedy jeszcze pewnie znaczna część Polaków liczyła na to, że może 2 tygodnie, może 3 tygodnie i pandemia będzie słabnąć. Natomiast widać bardzo wyraźnie, że jednak już liczymy się z perspektywą co najmniej 3 miesięcy funkcjonowania pandemii, a też nie jest pewne, czy jest to koniec.

Poszerzenie dla firm średnich, czyli tych zatrudniających do 49 osób. Oczywiście pamiętamy o tym pierwszym rozwiązaniu, że do dziewięciu osób również to funkcjonuje. Również wprowadza się pewne korekty i liczby ubezpieczonych, które zalicza się do zatrudnionych. Stąd też wielu przedsiębiorców, szczególnie małych przedsiębiorców, skorzysta, czyli wejdzie w próg do dziewięciu zatrudnionych. Niezwykle istotne rozwiązanie, o którym się bardzo mało mówi, to pożyczki na zachowanie miejsc pracy. Nie byłoby w tym oczywiście nic wielkiego, gdyby to były tylko pożyczki, ale to pożyczki, które będą umarzane pod warunkiem zachowania miejsc pracy. A więc to są tylko te najważniejsze formy pomocy przedsiębiorcom, którzy borykają się z problemami gospodarczymi związanymi bezpośrednio ze stanem epidemii w Polsce. Oczywiście jest tak, że prawdopodobnie życie będzie pokazywało dalsze rozwiązania i w razie rozwoju epidemii pewnie będą jeszcze inne korekty i poszerzenie zakresu pomocy z tego względu, że ważne jest, aby oprócz zachowania zdrowotnego, i to jest główny cel i ten cel realizuje się przez powszechną, narodową kwarantannę. Aby cel ochrony zdrowia, który jest realizowany w Polsce znakomicie, nie da się tego ukryć. Patrząc na statystyki zachorowań, śmiertelności w Polsce i w innych porównywalnych krajach europejskich, naprawdę jesteśmy dumni z tego, że te działania były podjęte tak wcześnie, tak przewidująco. I to jest najważniejsza część działań polskiego rządu. Ale oczywiście zarówno przedłużający się okres trwania epidemii, jak i zobowiązanie społeczeństwa do kwarantanny narodowej powodują niewątpliwe skutki gospodarcze. Te skutki gospodarcze rząd stara się w jak największym stopniu łagodzić, oczywiście biorąc też pod uwagę realność wydatków, chociaż poziom pomocy rzędu 10% PKB jest naprawdę poziomem bardzo istotnym. To jest ustawa, która daje realną pomoc przedsiębiorcom, równocześnie zapewniając stabilność finansów państwa. W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wnoszę o uchwalenie tej ustawy.

Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym. Informuję panie i panów posłów, że ustalam w tym punkcie limit 10 pytań dla klubów według następującego parytetu: Prawo i Sprawiedliwość - 5, Koalicja Obywatelska - 3, Lewica - 1, PSL-Kukiz15– 1, a także jedno pytanie dla koła. Jeżeli ktoś jeszcze z państwa klubów się nie zapisał, to bardzo proszę. Bardzo proszę, pani marszałek. Wysoka Izbo! Dobra ustawa, która daje pomoc, musi być prosta, dawać możliwość szybkiego działania i być zrozumiała. W tej ustawie z trudem można znaleźć pomysły, jak ludziom pomóc. Trzeba tłumacza, żeby ją zrozumieć. Zajmujemy się wszystkim, ale nie realną pomocą. Dotykam dwóch obszarów. Za 13 dni egzaminy ósmoklasistów. Nasza poprawka, która została odrzucona, dawała ministrowi szansę rozwiązania tego problemu. Tyle dni do egzaminów. Słowa, słowa ze strony rządu do dzieci, do młodzieży, do rodziców. Ta sprawa przez te wszystkie dni nie została podniesiona. Lekceważycie ją. Mówi się tyle, że kultura jest ważna. W tym projekcie nie ma ani jednego słowa o tym, jak pomóc temu przemysłowi, który w bardzo wielki sposób został dotknięty, bo tak naprawdę cały przemysł, cała branża (Dzwonek) kultury, ludzie kultury zostali zostawieni sami sobie. Proszę. Wysoka Izbo! Chciałam tylko zadać pytanie: Gdzie są te realne rozwiązania dla Polaków? Całą noc spędziliśmy nad projektem ustawy, w której wyłapywaliśmy - i to już było ewidentne - kolejne wrzutki. To jest po prostu kolejny TikTok, a nie realny pomysł dla Polaków. Bardzo rzetelnie apeluję, żeby rząd w tej chwili rzeczywiście skupił się na pracy, ponieważ my jako opozycja mamy obowiązek w tej chwili powiedzieć Polakom: Zostaliście sami. Te rozwiązania są daleko niewystarczające. Naprawdę weźmy się do roboty. Wszyscy. Z tego powodu bardzo proszę o to, żebyśmy wszyscy współpracowali.

Pan poseł Dariusz Klimczak, Koalicja Polska - PSL - Kukiz15. Wysoka Izbo! W czasie pandemii tarcza antykryzysowa powinna być jak arka dla wszystkich, która daje ratunek wszystkim. A co daje rząd? Rząd daje lichą tratwę dla nielicznych, dla tych mniejszych i lżejszych dla budżetu. Natomiast mam pytanie zasadnicze: Jak mogliście w ramach poprawek uchwalić prawo, które ułatwia zwalnianie pracowników w administracji? Jaki to jest przykład dla przedsiębiorców, którym mówicie: bądźcie silni, nie dajcie się, nie rozwalajcie własnych zespołów, a sami szykujecie się do odwrotu?

Jak pomaga rolnikom, którzy są producentami wczesnych warzyw? Jak pomaga wszystkim tym, którzy produkują kwiaty jednoroczne, rabatowe? To jest pytanie zasadnicze do ministra rolnictwa. Bo tarcza antykryzysowa (Dzwonek) to jedno, a te instrumenty, które dzisiaj ma minister, to jest druga sprawa. Pan poseł Zbigniew Konwiński, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Jeszcze przed wpłynięciem projektu rządowego do Wysokiej Izby Koalicja Obywatelska złożyła kilka projektów ustaw, które rzeczywiście wychodziły naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i pracowników, a także pracowników szeroko rozumianej ochrony zdrowia. Złożyliśmy projekt, aby zwolnić z ZUS-u również małe i średnie przedsiębiorstwa. Ale PiS jest przeciw. Złożyliśmy projekt, żeby ułatwić wypłatę odszkodowań dla przedsiębiorców, którzy ucierpieli wskutek decyzji rządu - szły im dobrze biznesy, dobrze prowadzili swoją działalność gospodarczą, ale to decyzja rządu spowodowała, że ich działalność została zawieszona. Niestety PiS jest przeciw. Zaproponowaliśmy także rozwiązanie, aby można było korzystać z konta VAT-owskiego, po żeby poprawić płynność działalności polskich przedsiębiorców. Niestety, szanowni państwo, PiS jest przeciw.

Niestety PiS jest przeciw. Złożyliśmy (Dzwonek) również wniosek, żeby obowiązkowo testować co tydzień pracowników służby zdrowia, farmaceutów. Niestety PiS jest przeciw.

Jest takie piękne słowo: empatia, czyli zrozumienie, współczucie. Tylko pytanie: Gdzie jest empatia w stosunku do pracownika firmy, która liczy 200 pracowników i która nie dostanie zwolnienia z ZUS, w związku z tym za moment 100 spośród nich zostanie zwolnionych? Gdzie jest empatia w stosunku do właścicielki trzech salonów kosmetycznych, która zatrudnia 10 pracowników, w związku z tym dostanie zwolnienie z ZUS tylko dla połowy z nich, dla pięciu? Gdzie jest empatia dla rodziców dwóch bliźniaków dziewięciolatków, którzy nie mogą zostać sami w domu, bo rozwaliliby ten dom, ale ona nie dostanie zasiłku, bo jej dzieci są już za duże? Gdzie jest empatia dla lekarzy, którzy mają maseczki tylko dzięki temu, że Łódź szyje dla medyków, czyli że obywatele szyją dla nich maseczki?

Ale moje pytanie brzmi: Jaki mamy plan na tę wojnę z wirusem tak naprawdę, jak zamierzamy ją wygrać? No, ja myślałem, że w maju to będziemy zwycięstwo świętować, a tu się okazuje, że rząd zaplanował klęskę. Jeśli planujecie taką ekstensywną walkę z tym wirusem przez bezterminowe zamykanie wszystkiego, to pytanie: Jak długo to ma potrwać? Za chwilę będą potężne deficyty we wszystkim, jeśli tak będziemy walczyć. Kupujemy sobie bardzo drogo czas, a nie przygotowujemy żadnej kontrofensywy. Nadal nie mamy żadnego ogłoszonego planu. Zwracam uwagę, że jeśli celem jest to, żeby utrzymywać zachorowania na poziomie kilkuset dziennie, to przejście choroby przez całą populację zajmie jakieś 200 lat.

Zamykam dyskusję. Bardzo proszę, panie premierze. Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Od kilku tygodni Polska i świat zmagają się z bardzo poważnymi wyzwaniami. Jest wielki kryzys epidemiczny, jest wielki kryzys gospodarczy, który nadchodzi. Polski rząd w sposób poważny i odpowiedzialny stara się rozwiązywać problemy Polaków. I od kilku tygodni słyszymy na tej sali inwektywy, insynuacje, epitety, nieprawdziwe stwierdzenia, mam nadzieję, że nie kłamstwa, a tylko mijanie się z prawdą. To bardzo przykre i bardzo smutne. Ja chciałem się odnieść tylko do kilku faktów, dzisiaj przez państwa przedstawianych właśnie jako fakty, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. nie wiem, z jakiego powodu pani mówi, że tarcza nie dotyczy ludzi kultury i sytuacji polskiej kultury. Od kilku tygodni dzień w dzień informujemy - na stronach ministerstwa można także to przeczytać, w moich wypowiedziach, w wypowiedziach bardzo wielu ludzi - co robimy dla ludzi kultury. Pani wyszła tutaj na mównicę i powiedziała, że nic nie zrobiliśmy i tarcza nie obejmuje ludzi kultury. To ja pani w takim razie podam tylko kilka faktów. Ludzie kultury działają w ramach działalności gospodarczej. Ludzie kultury bardzo często działają w oparciu o jednoosobową działalność gospodarczą albo też w oparciu o umowy cywilnoprawne. Tarcza przecież przedstawia konkretne fakty. Konkretne fakty, liczby, pieniądze. I w związku z tym polskie państwo wspomaga kulturę w tej kwestii. Wie pani doskonale, że już od poniedziałku działa nowy program ministra kultury, który został powołany dzięki tarczy antykryzysowej, który dotyczy kultury w sieci. Jest zapowiadany następny program, do którego się przygotowujemy, który będzie rekompensował straty. Są także realizowane w tej chwili odwołania w 32 programach ministra, które uwzględniają obecną sytuację.

I w tym kontekście faktycznie poważnej sytuacji na całym świecie, bardzo poważnej sytuacji w Polsce, tych wszystkich spraw, z którymi się musimy zmagać, a także poważnej sytuacji dla wszystkich branż, w tym dla ludzi kultury, pani wychodzi tutaj, pani marszałek, i mówi, że nic nie robimy. Są rozwiązania dotyczące także przemysłu filmowego, z którym pani była przez lata związana. Proszę sobie przeczytać tę ustawę, a nie kręcić głową. Ja pani mówię: została zmieniona definicja filmu, zostały zmienione także. Dobrze, że pani zgadza się ze mną. Jeszcze jedna kwestia, w zasadzie dwie kwestie, do których także chciałem się odnieść. Jeżeli chodzi o egzaminy, zapowiadaliśmy, że jutro będzie komunikat w tej kwestii. Apeluję do wszystkich uczniów, rodziców. Jak państwo wiecie, musieliśmy wprowadzić oczywiste obostrzenia. Dzięki nim nie mamy w tej chwili w Polsce 20 tys. czy więcej osób chorych, tylko mamy 5 tys., na szczęście. Szkoda, że 5 tys., bo to dużo, ale opanowaliśmy tę sytuację dzięki odpowiednim restrykcjom.

Mam nadzieję, że to nie było wystąpienie motywowane złą wolą, a brakiem informacji. W Polsce są 824 domy pomocy społecznej. W 14 domach pomocy społecznej faktycznie mamy problem z epidemią, z szerzeniem się epidemii. Dotyczy to nie setek, a 169 osób, które są chore. To jest o 169 osób za dużo (Dzwonek), ale to naprawdę nie jest sytuacja, którą można z dnia na dzień zlikwidować, i to jest nasz wspólny ból. Codziennie spotyka się zespół zarządzania kryzysowego i codziennie, także dzisiaj, rozmawiamy na temat sytuacji w domach pomocy społecznej. W tej chwili państwo jest tam obecne: z pomocą, ze wsparciem i z nadzorem. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm skierował ten projekt do Komisji Finansów Publicznych w celu przedstawienia sprawozdania. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę.